Wznawiam obrady.

Stwierdzam kworum. Właściwa komisja przedłożyła sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, druk nr 2082. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 2079-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Michała Jacha o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek! Panowie i Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o obronie Ojczyzny, druk nr 2052. Komisja Obrony Narodowej proponuje przyjąć 13 poprawek, odrzucić 52 poprawki.

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 2079. Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności. Głosujemy. Kto jest za

Sejm poprawkę odrzucił.

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za 4. poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o ich odrzucenie.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił.

Kto się wstrzymał?

Kto jest za przyjęciem 8. poprawki? Kto jest przeciw?

Kto jest za przyjęciem 9. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeszcze nie zakończyłam głosowania. U kogo nie działa? To proszę zmienić miejsce. Działa, pani poseł?

Kto jest za 10. poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto jest za przyjęciem 11. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto jest za przyjęciem 13. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za przyjęciem 14. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał.

Sejm poprawkę przyjął. Kto jest za 15. poprawką? Kto jest przeciw?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Wszyscy byli za. Sejm poprawkę przyjął.

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

371 - za, nikt nie był przeciw, 84 się wstrzymało. Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął.

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto jest za 55. poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Kto jest za 58. poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy nad 60. poprawką. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2079, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o obronie Ojczyzny. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 18. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Obrony Narodowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (druki nr 2081 i 2082) Proszę pana posła Krzysztofa Tchórzewskiego o przedstawienie sprawozdania komisji.

Wysoki Sejmie! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Obrony Narodowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, druk nr 2081. Marszałek Sejmu skierowała w dniu 11 marca 2022 r. uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Obrony Narodowej do rozpatrzenia. Została zgłoszona jedna poprawka.

W związku z tym wysokie komisje rekomendują, żeby tę poprawkę przyjąć. Przypominam, że Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu, uważa się ją za przyjętą. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Ja nie wiem, co za. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 11 marca br.